Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Spraw Zagranicznych - godz. 9, - do Spraw Energii i Skarbu Państwa - godz. 10.30. Informuję, że na podstawie art. 198a ust. 2 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o kontynuacji 10. posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe.

Panie pośle, może po tym punkcie, bo i tak nie będziemy ich teraz. Bardzo proszę, niech pan przedstawi. Szczęść Boże! Wysoka Izbo! Wniosek o ogłoszenie przerwy celem odbycia posiedzenia Prezydium Sejmu, by zanim Sejm podejmie pracę, wyciągnąć wnioski z wczorajszego skandalicznego zachowania członków Prezydium Sejmu, którzy nadużyli swoich uprawnień, przekroczyli je, jednocześnie nie dopełnili swoich obowiązków. Czas najwyższy, zanim zaczniemy spotykać się na posiedzeniach Komisji Etyki Poselskiej czy ciągać po sądach, panie marszałku, położyć kres tym manifestacjom brutalnego prostactwa, ośmielę się zdiagnozować, które mieliśmy tutaj w całym cyklu w dniu wczorajszym. Proszę, szanowne Prezydium, ogarnijcie się, zanim dopuścicie się poważniejszych jeszcze przekroczeń prawa i regulaminów. Panie pośle, zastanowię się, czy wypowiedź pana posła kwalifikuje się do komisji etyki i ukarania.

Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami trzynaste emerytury będą rokrocznie wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu. Trzynasta emerytura będzie stanowić potężne wsparcie finansowe dla świadczeniobiorców otrzymujących minimalne emerytury i renty. Stąd też kieruję do pani minister swe pytania. Ilu Polaków obecnie otrzymuje emeryturę lub rentę w najniższej wysokości? Czy osoba, która nabędzie prawa emerytalne w kwietniu 2020 r., również otrzyma trzynastą emeryturę? I chciałem, aby pani minister potwierdziła to, o co pyta wielu emerytów i rencistów, czyli gwarancje wypłat w obecnej wysokości emerytur i rent. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana ministra Stanisława Szweda. Bardzo proszę.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Dziękuję za to pytanie. Zanim odniosę się do tej głównej treści pytania dotyczącej dodatkowego świadczenia zwanego trzynastą emeryturą, to może podam też kilka informacji dotyczących w ogóle sytuacji osób starszych i tych działań, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, jeśli chodzi o wsparcie dla emerytów i rencistów. Myślę, że takim najważniejszym momentem, w którym dokonaliśmy istotnej zmiany, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne, była kwestia podniesienia minimalnej emerytury. To był wzrost o ponad 13%. To spowodowało, że ta najniższa emerytura zaczęła rosnąć w szybszym tempie, niż to było dotychczas, jeśli chodzi o wzrost wskaźnika emerytalnego, i to było też ważne na wszystkich etapach waloryzacji.

To spowodowało, że ten wskaźnik, który zawsze był określany jako wskaźnik procentowy, zamieniliśmy na wskaźnik wzrostu emerytur i rent, na wskaźnik kwotowo-procentowy.

Dzisiaj minimalna emerytura wynosi 1200 zł brutto, tak jak już pan poseł powiedział, 981 zł netto, a najniższa emerytura netto to jest 1025 zł. Całkowity koszt tegorocznej waloryzacji to było ponad 9 mld zł.

Jeśli chodzi o kwestię związaną z trzynastą emeryturą, to, o co pan poseł pytał, dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastą emeryturę, która jest wpisana na stałe do ustawy, która będzie corocznie obowiązywała, to ona jest wypłacana w kwocie najniższej emerytury, czyli 1200 zł brutto, i dotyczy wszystkich emerytów, rencistów, osób, które są na świadczeniach kompensacyjnych, na świadczeniach przedemerytalnych, także emerytów, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie, jak również tych emerytów, którzy są w służbach mundurowych.

Co jest ważne, ta dodatkowa trzynasta emerytura nie ma wpływu na inne świadczenia, czyli doliczamy do dochodu, zarówno jeśli chodzi o dodatki, zasiłki czy ulgę rehabilitacyjną.

Teraz uzupełniające pytanie zadaje pan poseł Marek Suski. Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Wielu seniorów w związku z koronawirusem ma obawy, czy nie zabraknie pieniędzy. I tu jest pytanie o to, czy mamy pełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o emerytury i wypłaty trzynastek, bo ludzie są zaniepokojeni, że w związku z tym kryzysem może być jakiś problem. Bardzo proszę o zapewnienie naszych rodaków, że nie ma z tym problemu. Ponownie odpowiada pan minister. Oczywiście jeszcze raz chcę podkreślić, że nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o wypłatę trzynastej emerytury. W tegorocznym budżecie środki są zapewnione, tak jak powiedziałem, ponad 11 mld zł zarówno z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z KRUS-u, jak również w służbach mundurowych, czyli bezpośrednio z budżetu państwa. Zagrożenia, jeśli chodzi o wypłatę trzynastych emerytur, nie ma. Tak że emeryci mogą być spokojni o to, że w tym roku je dostaną, dostaną również w przyszłym roku. Ona jest na stałe wpisana do ustawy i będzie realizowana, tak samo jak program „Rodzina 500+” Nie, to są te działania, które podjęliśmy, które dzisiaj w tej naszej bardzo trudnej sytuacji odpowiadają też na zapotrzebowanie naszych rodaków. To wsparcie jest. Na program 500+ mamy ponad 100 mld zł, które trafiły do polskich rodzin.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował tę politykę, aby wspierać w tych trudnych momentach również polskie rodziny. Bardzo dziękuję. Zauważyłem, że klub Lewicy przekroczył limit osób na sali. Wysoka Izbo! Chciałam tylko poprosić pana marszałka o sprawdzenie kworum, bo tak naprawdę nie wiemy, czy mamy kworum, a rozpoczęliśmy obrady. Nie było w tej kwestii sprawdzenia. Dziękuję. Sprawdzimy kworum przed głosowaniem. Bardzo proszę, przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Marta Wcisło, Michał Szczerba, Barbara Nowacka i Monika Rosa z klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie sytuacji placówek stałego pobytu dla osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Bardzo proszę. Pierwsze pytanie zadaje pani poseł Marta Wcisło. Wysoka Izbo! Podstawowym obowiązkiem państwa demokratycznego jest szczególna dbałość i troska o osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Mówi o tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 68 ust. 3. Tak jednak się nie dzieje. W naszym kraju mamy na obecną chwilę blisko 8 tys. chorych, w tym najwięcej osób starszych, osób z grupy najwyższego ryzyka, podopiecznych domów pomocy społecznej, którzy chorują grupowo, tak jak miało to miejsce we Włoszech, w Hiszpanii czy innych krajach Europy. Był czas na to, aby się do tego przygotować. Trzeba było i można było temu zapobiec. Rząd zapewniał, że jesteśmy przygotowani na walkę z koronawirusem, że wyprzedzamy Europę i że Europa może brać z nas przykład. Tymczasem rozgrywają się dramaty, ludzkie dramaty osób starszych i chorych w domach pomocy społecznej. Można było do tego nie dopuścić, gdyby rząd w odpowiedniej chwili wprowadził procedury, testy, środki ochrony osobistej. Można było nie dopuścić do tego, co dzieje się dzisiaj w Jakubowicach, Skarżysku-Kamiennej, Stalowej Woli, Psarach i w wielu innych domach pomocy społecznej. Nie jest to wina, szanowni państwo, zarządzających czy personelu, bo oni robią, co mogą, ale zostali sami, zostali bez pomocy. Do dziś nie ma środków ochrony osobistej i testów, do dziś nie ma procedur. Rząd nie ma czasu na to, aby zająć się osobami z grupy najwyższego ryzyka, mimo że byliśmy zapewniani, że jesteśmy przygotowani do walki z koronawirusem, że mamy wszystko. Pani minister, dlaczego? Dlaczego personel domów pomocy społecznej nie ma środków ochrony osobistej? Wczoraj to sprawdzałam. Dlaczego nie ma szybkich testów?

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Obowiązkiem państwa jest zadbać o osoby starsze, potrzebujące pomocy i osoby niepełnosprawne, rzeczywiście zadbać, a nie mówić tylko o tym, że dbamy, i nie uprawiać retoryki, która jest zbędna i niepotrzebna. Szanowni Państwo! Od samego początku, kiedy epidemia w naszym kraju została odnotowana, od pierwszego dnia zostały wprowadzone procedury. Krok po kroku odniosę się do liczb, procedur i całej działalności. Przypomnę, że to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wspomaga samorządy w realizacji ich zadań własnych. Opieka społeczna to jest zadanie własne samorządu. Mamy 824 domy pomocy społecznej, które są prowadzone przez samorządy i właśnie tym samorządom pomaga rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Ministerstwo rodziny poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje zalecenia, polecenia, które wojewodowie przekazują do jednostek samorządu terytorialnego, i są one wprowadzane w życie. Pierwsze procedury zostały wprowadzone 13 marca. A więc, pani poseł, proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Tak jak mówimy i mówić będziemy, i potwierdzamy to w działaniu, przede wszystkim wiarygodność jest podstawą naszego działania. Wiarygodność i odpowiedzialność za losy wszystkich Polek i Polaków, a w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych. Każdego dnia to czynimy. Jeśli chodzi o wszystkie procedury, poczynając od zamknięcia domów pomocy społecznej, a także całodobowych ośrodków, które notabene są prowadzone przez osoby fizyczne jako podmioty, wszędzie z naszej strony poszły rekomendacje co do tego, jak należy postępować w sytuacjach kryzysowych.

Przejdę teraz do konkretów, skąd tylu chorych i jak to wygląda, i może zderzymy mity z rzeczywistością. Szanowni Państwo! Mamy 824 domy pomocy społecznej.

Domy zostały wyposażone w przywołane instrukcje, środki ochrony osobistej, a także rząd przekazał dodatkowe środki. I to nie jest ostatnie wsparcie. Każdego dnia - dosłownie każdego dnia - monitorowana jest sytuacja i podejmowane są decyzje.

Tak jak zadbaliśmy o to, żeby była tarcza antykryzysowa, tak przed tym działaniem zostały wprowadzone wszelkie procedury, aby przede wszystkim zabezpieczyć, wesprzeć te organy, które odpowiadają za prowadzenie tych placówek.

Jeżeli byśmy chcieli te liczby przekładać na procenty, to one są małe, ale to nie o to chodzi. Najważniejszy jest człowiek i jego wsparcie.

Bardzo proszę. Państwo, które nie potrafi chronić najsłabszych i najbardziej bezbronnych, nie potrafi chronić nikogo. Mówimy o domach pomocy społecznej, których jest 875 - to są dane NIK-u - mówimy o 620 placówkach całodobowej opieki prowadzonej w ramach działalności, ale również, pani minister, i pani tego nie zauważa, mówimy o 124 placówkach opieki działających bez zezwoleń wojewodów. Chciałbym panią wezwać do odpowiedzi na pytanie, jakie działania wobec tych nielegalnych placówek, o których pani wie i wojewodowie wiedzą, państwo wykonaliście. Personel boi się pracować w DPS-ach, bo rząd skąpi testów. Teraz praca w DPS-ach przypomina po prostu rosyjską ruletkę. To, co dzieje się na Mazowszu, to jest niebywały skandal. Bobrowiecka, Tomczyce, Niedabyl, Rusiec. Wojewoda Radziwiłł kieruje do pracy (Dzwonek) matkę karmiącą 5-miesięczne dziecko, a następnie nakłada na nią karę finansową. Zróbcie porządek z panem wojewodą Radziwiłłem. Ten człowiek zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu na Mazowszu. Dziękuję. Bardzo proszę, ponownie odpowie na pytanie pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Pośle! Posługujemy się liczbami, które niestety nie są prawdziwe. To jest fakt.

Odniosę się do Mazowsza, które pan poseł tutaj tak pięknie przywołał, mówił o sytuacji w Niedabylu. Właśnie Niedabyl pokazuje opanowanie sytuacji przez wojewodę, czyli wsparcie przede wszystkim podmiotu, który jest organem prowadzącym dla tego domu pomocy społecznej.

A więc, panie pośle, nie opowiadajmy tutaj rzeczy, które są nieprawdziwe. Wojewoda mazowiecki pan dr Konstanty Radziwiłł podjął słuszne działania. Jeżeli personel choruje czy brakuje personelu, ma uprawnienia do tego, aby nakazać pracę, wyznaczyć osoby do pracy w domach pomocy społecznej. Pani poseł. Mam listę osób, które pan wojewoda skierował do pracy. Cóż te osoby zrobiły od razu? Wzięły zwolnienie lekarskie, L4.

Decyzje pana wojewody były decyzjami słusznymi i przede wszystkim miały zabezpieczyć obydwie strony. A więc każda sytuacja jest indywidualna. Tak jak powiedziałam przed chwilą, wszystkie te placówki zostały wyposażone w sprzęt ochrony osobistej, zostały wyposażone w dodatkowe środki.

Pani Minister! Dobrze, ale to poprosiłbym, panie marszałku, o informację na piśmie. Medycy to nie są takie worki kartofli, które można przestawiać z miejsca na miejsce. Trzeba przestrzegać prawa i trzeba działać zgodnie z trybem, który jest wskazany w ustawie o zakażeniach. Nie można kierować do pracy osób powyżej 60. roku życia. Wojewoda Radziwiłł takie osoby kieruje do pracy, a jednocześnie nakłada na nie 5-tysięczne kary. Wojewoda mazowiecki Radziwiłł kieruje do pracy matki karmiące 5-miesięczne dzieci. Nakłada na nie kary. Nie ma do tego prawa, ponieważ osoba opiekująca się małoletnim dzieckiem nie może być kierowana do pracy.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Robert Obaz, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Nawiązując do wczorajszych wystąpień, gdzie raz po raz właśnie z tej mównicy akcentowano, że miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek do życia - tak mówili posłowie PiS - pytam państwa w imieniu niepełnosprawnych, starszych i schorowanych pensjonariuszy DPS-ów w Niedabylu, Tomczycach czy Skarżysku-Kamiennej, pytam, bo prawem opozycji jest dzisiaj pytać, co rząd zrobił dla tych najsłabszych, często pozbawionych nie tylko zdrowia, ale też godności, na jaką zasługuje każdy z nas. Ostatnie informacje z Ministerstwa Zdrowia o rosnącej liczbie zagrożonych pensjonariuszy domów pomocy społecznej stawiają pod znakiem zapytania ich los, bezpieczeństwo, a nade wszystko zdrowie. DPS-y nie są zakładami opieki zdrowotnej, dlatego też nie mogą skorzystać z zasobów posiadanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, nie tak dawno kontrolowanych przez posłów Lewicy.

Jakie działania zainicjowały inspektoraty sanitarne i wojewodowie w zakresie profilaktyki rozpoznawania objawów u pensjonariuszy i wdrożenia zabezpieczeń dezynfekcyjnych? Czy podjęto działania w celu wyposażenia tych placówek w wystarczające ilości środków ochrony osobistej? Po trzecie, jakie działania zainicjowano, by mieszkańcy zgłaszający objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem byli poddawani izolacji oraz czy izolacja ma miejsce w obrębie placówki, w której przebywają pensjonariusze, czy też w warunkach szpitalnych? Jakie działania zostały zainicjowane, by w placówkach były opracowane i wdrożone procedury na okoliczność wysokiego stopnia absencji wśród personelu placówki?

Bardzo proszę.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Seniorzy są szczególną grupą, która jest w sposób szczególny narażona na zakażenie koronawirusem. Z tego tytułu rząd podejmuje szczególne działania kierowane właśnie do tej grupy, aby ją maksymalnie chronić przed infekcją, a także przed niebezpiecznym przebiegiem tejże choroby.

Uzgadniając procedury, przygotowujemy stosowne wytyczne, stosowne wskazówki, w jaki sposób należy postępować, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa w całodobowych zakładach opieki społecznej czy opieki zdrowotnej. Zostały wydane konkretne zalecenia, konkretne procedury. Od początku trwania tej epidemii te zalecenia są publikowane na stronach głównego inspektora sanitarnego i na stronach ministra zdrowia. Oprócz tego w przypadku podmiotów leczniczych, jakimi są zakłady opiekuńczo-lecznicze, są przekazywane w systemie zarządzania informacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczególny nacisk kładliśmy i kładziemy nadal na szkolenie personelu. Konsultanci wojewódzcy, konsultanci krajowi zostali zobligowani do nadzoru nad przebiegiem procesu szkolenia personelu w taki sposób, aby eliminować te zachowania, które mogą skutkować transmisją wirusa, i wyposażyć pracowników maksymalnie w wiedzę, umiejętności posługiwania się środkami ochrony osobistej, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Minister zdrowia w marcu wydał również komunikat, w którym zaleca, aby personel medyczny, który jest szczególnie narażony na zakażenia, nie transmitował tego wirusa do podmiotów, szczególnie DPS-ów czy też zakładów opiekuńczo-leczniczych. Zwróciliśmy się do personelu medycznego, aby maksymalnie ograniczył miejsca świadczenia pracy. Jeżeli chodzi o konkretne zabezpieczenie tych podmiotów, o których mówimy, chcę podkreślić, że na wniosek ministra rodziny minister zdrowia wydał decyzję o kilkakrotnym przekazaniu środków ochrony osobistej, jak również płynów dezynfekcyjnych do domów pomocy społecznej.

Na bieżąco oczywiście te środki są przekazywane, w zależności od wniosków, które spływają do wojewodów. Jeżeli chodzi o kwestię wykonywania badań, badania są wykonywane na podstawie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, która wyraźnie wskazuje, jak powinien być zdefiniowany przypadek kwalifikujący do wykonywania badań. W tej chwili badania są wykonywane osobom, które na podstawie wywiadu epidemiologicznego wykazują ryzyko kontaktu z osobą, która jest nosicielem koronawirusa. Również badania wykonywane są osobom, które mają objawy świadczące o tym, że mogło dojść do zakażenia koronawirusem. Badania są wykonywane również osobom przebywającym na kwarantannie. Jeżeli mieszkaniec domu pomocy społecznej czy zakładu opiekuńczo-leczniczego spełnia te przesłanki, ma wykonywane tego typu badanie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał stosowne zarządzenie, na mocy którego zarówno pracownicy podmiotów leczniczych, jak i pracownicy medyczni zatrudnieni w DPS-ach mogą mieć wykonywane badania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Te badania mogą przeprowadzać podmioty lecznicze, które mają stosowne laboratoria i są wpisane na listę wojewodów. Reasumując, chciałabym powiedzieć, że podjęliśmy wszelkie działania, żeby wyposażyć w środki ochrony osobistej, przeszkolić, jak również wprowadzić standardy organizacji pracy, które mają na celu zmniejszenie emisji koronawirusa. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę uściślić. Mówimy o ponad 80 tys. ludzi, o pensjonariuszkach i pensjonariuszach w DPS-ach, tysiącach osób w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, o personelu, o tych osobach, o które ani ten rząd, ani poprzednie rządy po prostu nie dbały. Chciałabym usłyszeć konkretny plan pomocy i zabezpieczenia tych podopiecznych i pracujących tam osób. Pani Minister! Dramatycznie brakuje tam opiekunek, pielęgniarek i lekarzy. Pani minister, na jakich zasadach środki ochrony osobistej są tam przekazywane? Czy znacie państwo środki, potrzeby konkretnych ośrodków? Ostatnio wojewoda przekazał jednemu z małopolskich DPS-ów kombinezony na 3 dni. Czy to jest wystarczająca pomoc? Jaka jest ścieżka uzyskania tej pomocy? Czy ministerstwo przewiduje także ewakuację zarażonych, zakażonych podopiecznych? Potrzebujemy realnego planu pomocy (Dzwonek), konkretnych instrukcji, a nie umywania rąk. Bardzo proszę. Szanowna Pani Poseł! Ja już przedstawiłam działania rządu w zakresie wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej czy w zakładach opiekuńczo-leczniczych, natomiast chcę uzupełnić, że jeżeli chodzi o standard opieki medycznej, to jest on określony w stosownych aktach prawnych. Jeżeli chodzi o DPS-y, mieszkańcy DPS-ów, każdy z tych mieszkańców, tak jak każdy z nas, ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie poprzez wskaźnik 3 razy wyższy niż w przypadku pozostałych obywateli. W związku z sytuacją epidemiczną prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się do lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych o objęcie szczególną opieką mieszkańców właśnie domów pomocy społecznej. Wdrożono standardy postępowania polegające na takim dwukrotnym triażowaniu mieszkańców domów pomocy społecznej, tzn. analizie, badaniu temperatury, liczby oddechów dwa razy dziennie i jeszcze obserwacji w kierunku innych objawów, które mogą sugerować zarażenie koronawirusem, chodzi o monitorowanie stanu zdrowia. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lekarz, personel domu pomocy społecznej zna doskonale standard, czyli dzwoni do lekarza rodzinnego, który podejmuje stosowane działania. W związku z sytuacją epidemiczną prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadził możliwość finansowania świadczeń za pomocą technik telekomunikacyjnych, czyli teleporady. Dzięki temu mieszkańcy domów pomocy społecznej mogą na bieżąco komunikować się z osobami, które się nimi opiekują. Jeżeli chodzi o dostarczanie sprzętu, to jeszcze raz chcę pani poseł przypomnieć, że z Agencji Rezerw Materiałowych na bieżąco są przekazywane środki do wojewodów i wojewodowie na podstawie analizy zapotrzebowania składanego przez poszczególne podmioty na bieżąco dostarczają je do konkretnych podmiotów leczniczych. Tak że dbamy o to, aby wojewodowie dysponowali tymi środkami, natomiast decyzja o skierowaniu odpowiedniej partii środków dezynfekcyjnych czy materiałów, czy środków ochrony osobistej podejmowana jest na poziomie wojewody. Szanowni Państwo!

Przechodzimy do kolejnego pytania. Bardzo proszę, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie sytuacji w domach pomocy społecznej. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie powstało na kanwie sytuacji, jaka miała i ma miejsce w domu pomocy społecznej w Drzewicy w województwie łódzkim. W tym domu pomocy społecznej bardzo szybko doszło do bardzo licznych zakażeń zarówno wśród podopiecznych, jak i wśród pracowników domu pomocy społecznej.

W wyniku tego wojewoda łódzki nakazem pracy oddelegował część, m.in. panie pielęgniarki ze szpitala powiatowego w Opocznie, do pracy w tym DPS-ie. Jak się okazało, tych pań pielęgniarek miało pracować w sumie sześć. Ta sytuacja trwała od Wielkiego Czwartku do przedwczoraj, natomiast w dniu wczorajszym i dniu dzisiejszym trwa ewakuacja domu pomocy społecznej. Ze względu na to, że pani minister niedawno, przed chwilą mówiła, odpowiadając na pytania posłów Koalicji Obywatelskiej, że ministerstwo wysłało rekomendacje co do postępowania w określonych sytuacjach, np. w DPS-ach, rozumiem, wojewodom, chciałbym zapytać: Jakiego rodzaju rekomendacje ministerstwo wskazuje w takiej sytuacji, kiedy teoretycznie funkcjonuje dom pomocy społecznej, nie ma tam określonej kadry medycznej, opieki pielęgniarskiej, nie ma zwykłych pracowników, którzy się zaopiekują podopiecznymi, i zapada po kilku dniach decyzja o ewakuacji? Czy takie, tego typu ewakuacje nie powinny odbywać się natychmiast, kiedy nie ma kadry pracowniczej? Mam także pytanie, czy ministerstwo, czy rząd pracuje nad modyfikacją (Dzwonek) przepisów i procedur, które pozwoliłyby na uniknięcie takich sytuacji, oraz w jaki sposób wojewodowie oceniają, dokonują oceny osób, które mają dostać nakaz pracy i być delegowane do pracy w określonych miejscach. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani minister Barbara Socha. Bardzo proszę.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Sytuacje są bardzo, bardzo różne i musimy w domach pomocy społecznej reagować bardzo elastycznie.

Przeprowadzono również różne testy. Jutro, przepraszam, co ja mówię, przepraszam.

Tam mają dobrą opiekę i są doskonale, tzn. w miarę możliwości i, mam nadzieję, bardzo skutecznie, bardzo słusznie objęci opieką.

Oni na bieżąco relacjonują nam to, co się dzieje w ich województwach, i na bieżąco podejmujemy takie decyzje, jakie są najlepsze - najlepsze - dla pracowników domów pomocy społecznej i dla personelu. W zależności od tego, gdzie co jest potrzebne, będziemy dostarczać środki ochrony osobistej, będziemy starać się pozyskać nowy personel, tam gdzie jest taka potrzeba. A jeżeli będą bardzo trudne sytuacje, to będziemy ewakuować mieszkańców do szpitali, bo tam będą mieli dobrą opiekę. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Chciałbym odnieść się do sprawy przywołanego już tutaj dzisiaj wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który powołując się na art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, chyba nie znając do końca okoliczności, które zwalniają zgodnie z tą ustawą osoby z obowiązku takiego świadczenia, próbował przymusić pracowników środowiskowego domu społecznego w Łychowskiej Woli do pracy w domu opieki społecznej w Tomczycach, a następnie ukarał ich karami w wysokości 5 tys. zł. Szanowni państwo, wydaje mi się, że kogo jak kogo, ale wojewodę trzeba byłoby rozliczyć ze znajomości prawa. Bardzo proszę o to, pani minister. Ponownie odpowiada. Bardzo proszę. Szanowny Panie Pośle!

Mamy zdiagnozowaną sytuację indywidualną każdego przypadku, w którym zostały te nakazy wydane.

Od samego początku, powtórzę, zostały wdrożone procedury, działamy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Ministerstwem Obrony Narodowej.

W piątek wieczorem wojewoda. Przeanalizowaliśmy propozycję wojewody, że ewakuacja będzie rzeczą najlepszą, na taką decyzję się zgodziliśmy. Każdego dnia to monitorujemy.

Bardzo dziękuję, pani minister. Panie pośle Nitras, pani marszałek nie zgodziła się na pana udział w posiedzeniach na tej sali.

Proszę łaskawie opuścić salę. Kolejne pytanie. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zadaje pytanie w sprawie działań, jakie podejmuje Ministerstwo Zdrowia w celu zapewnienia odpowiedniej ilości środków ochrony dla szpitali. Jako pierwsza pani poseł Anita Czerwińska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W ciągu ostatnich tygodni możemy zaobserwować lawinowy wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Uwzględniając te statystyki, chciałam zapytać, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza zabezpieczyć szpitale, przychodnie i ich pracowników przed zakażeniem. Zadam też pytanie uzupełniające: Czy są planowane duże zakupy środków ochrony osobistej i ich dystrybucja do wszystkich szpitali w kraju? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! Ochrona personelu medycznego jest podstawową troską ministra zdrowia. Dlatego też od początku podejmujemy szereg działań mających na celu ochronę wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, ale również innych pracowników ochrony zdrowia. Nie jest tajemnicą, że od wielu lat borykamy się z problemami kadrowymi w ochronie zdrowia.

Dopiero w ostatnich latach podjęliśmy konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji kadrowej. Zwiększyliśmy liczbę szkół kształcących pielęgniarki, lekarzy, poprawiliśmy system wynagrodzeń. Dzięki temu udało się uzyskać pewną poprawę, jeżeli chodzi o kadry medyczne, ale w obliczu epidemii ta ilość kadry jest niewystarczająca. Dlatego też szczególne działania są kierowane do przedstawicieli zawodów medycznych. Chcemy ich maksymalnie chronić. Środki ochrony osobistej stanowią podstawowy element tej ochrony. To są bardzo ważne elementy w ochronie poszczególnych pracowników. Jeżeli chodzi o dostarczanie środków ochrony osobistej, to chcę podkreślić, że już w lutym pierwsze dostawy zostały skierowane do szpitali jednoimiennych. Jak państwo wiecie, w skali kraju mamy 19 szpitali jednoimiennych, które zostały wskazane jako podmioty zajmujące się tylko i wyłącznie pacjentami zakażonymi koronawirusem, i tam w pierwszym rzędzie zostały skierowane dostawy - dostawy środków ochrony osobistej, czyli odpowiednia liczba rękawic, gogli, fartuchów, kombinezonów, maseczek itd. Kolejne dostawy były kierowane sukcesywnie. O dostawach do szpitali jednoimiennych czy do oddziałów zakaźnych decydował minister zdrowia, wydając stosowne polecenia skierowane do Agencji Rezerw Materiałowych. Aktualnie minister zdrowia dysponuje zasobami pozyskanymi w drodze zakupów prowadzonych przez Biuro Administracyjne Ministerstwa Zdrowia. Dysponujemy również środkami, które pozyskaliśmy w trybie darowizn, udostępnianymi z rezerw strategicznych na rzecz ministra zdrowia.

Pozyskane zasoby są gromadzone w wybranych magazynach, składnicach rezerw materiałowych, które pełnią funkcję operatora logistycznego dla dostaw środków ochrony medycznej. Jednocześnie Agencja Rezerw Materiałowych nadal działa w granicach swoich uprawnień ustawowych i dokonuje zakupów w ramach odtwarzania udostępnionych wcześniej rezerw strategicznych. Tak jak wspomniałam, na bieżąco są uzupełniane dostawy do szpitali jednoimiennych, ale również przekazujemy odpowiednią partię, odpowiednią ilość środków dla wojewodów, którzy w dużej mierze decydują o dystrybucji tych środków do pozostałych podmiotów leczniczych. Od początku trwania tej epidemii przekazaliśmy właściwie ponad 585 tys. kombinezonów ochronnych.

Jeżeli chodzi o rękawice ochronne - ponad 16 mln. Jeżeli państwo sobie życzycie, to możemy państwu przekazać szczegółowe dane według poszczególnych rodzajów asortymentu środków ochrony osobistej. Chciałabym podkreślić, że na bieżąco są uzupełniane te zapasy, dystrybucja trwa różnymi kanałami, m.in. dużą rolę odgrywają tutaj Wojska Obrony Terytorialnej, odgrywa Poczta Polska, która bezpośrednio dostarcza te środki ochrony osobistej (Dzwonek) do konkretnych podmiotów.

Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Panie pośle, konsultowałem to z panią marszałek i pani marszałek wyraziła zgodę, żeby pan wyjątkowo wystąpił teraz w tym pytaniu. A więc pierwsze pytanie zadaje pan poseł Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska. Ja nie zadaję pytania wyjątkowo, tylko korzystam ze swojego prawa, a pan ani pani marszałek nie macie prawa ograniczać mi prawa wejścia na salę plenarną.

Wprowadziliście największe ograniczenia co do możliwości poruszania się przez Polaków w Europie włącznie z tym, że pozamykaliście lasy i parki.

Dzisiaj doprowadziliście państwo przez brak testów do sytuacji, w której polskie szpitale, zamiast być źródłem leczenia i pewnej nadziei, stały się źródłem pandemii. To w szpitalach dzisiaj najłatwiej się zarazić, dlatego że państwo nie testowaliście pracowników służby zdrowia, nie daliście im podstawowych instrumentów do walki z pandemią. Pozwoliliście państwo na to, żeby pracownicy służby zdrowia w tym trudnym okresie pracowali w kilku różnych szpitalach, przenosząc zarazę z jednego szpitala do drugiego. I oskarżam państwa, że to państwo jesteście dzisiaj przyczyną tego, że nie wiemy, ilu mamy zarażonych, bo najmniej badamy, a jednocześnie tego, że ta pandemia właśnie w szpitalach najbardziej się rozprzestrzenia. Nie zadbaliście państwo o podstawowe rzeczy, właśnie o testy. Natomiast ograniczenia, które wprowadziliście państwo, spowodowały, że polska gospodarka według danych rządowych dziennie - powołuję się na ministrów tego rządu - traci 8 W sytuacji, w której dzięki badaniu, dzięki testom takie kraje jak Niemcy, Dania, Czechy otwierają sklepy i uruchamiają swoją gospodarkę, jedyne, co macie nam do zaproponowania, to otwarcie lasów. Trzeba jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie ludzi zdrowych, a eliminować, izolować ludzi, którzy są zarażeni. Dziękuję. Odpowiedzi udziela sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko. Szanowni Państwo! Chciałabym na wstępie sprostować te nieprawdziwe wypowiedzi pana posła, ponieważ w Polsce testy wykonywane są zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

A więc każda osoba, która na podstawie wywiadu epidemiologicznego wykazuje prawdopodobieństwo kontaktu z osobą, która jest zarażona koronawirusem, jest kwalifikowana do testów. Każda osoba, która manifestuje objawy świadczące o tym, że mogła mieć kontakt z koronawirusem, może być zakażano i rozpoczyna się już wstępny proces choroby, również ma wykonywane testy. Każda osoba, która przebywa w kwarantannie, również ma wykonywane testy. Takie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Minister zdrowia podjął decyzję o zabezpieczeniu maksymalnej liczby testów, które są niezbędne do wykonywania testów dla naszych mieszkańców. Obecnie w naszym kraju wydolność zakładów diagnostyki laboratoryjnej jest na poziomie ok. 20 tys. testów dziennie. Obecnie wykonujemy tych testów - informacja z wczorajszego dnia - ponad 8 tys. dziennie. W poprzednim tygodniu wykonywaliśmy ok. 11 tys. dziennie. Te osoby nie mają ograniczonego dostępu do testów. Jeżeli chodzi o testowanie pracowników ochrony zdrowia, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, na gruncie którego każdy szpital, który posiada właściwe laboratorium diagnostyczne, może wykonywać badania zarówno dla pacjentów, jak również dla pracowników. Te badania są w 100% finansowane jako odrębny produkt przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A więc są ustalone poszczególne ścieżki, poszczególne możliwości realizowania tych testów. Jeżeli chodzi o dostępność testów i możliwości ich wykonywania, to tak jak państwu mówiłam, możliwości dzienne to jest ok. 20 tys. Do tej pory zostało wykonanych w Polsce ponad 153 tys. testów. Jeżeli chodzi o materiał do testowania, czyli testy, które zapewnialiśmy z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych, to są to następujące liczby. Do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i szpitali zostało przekazanych ponad 313 tys. testów, 223 tys. izolacji, 83 300 wymazówek z podłożem, 48 tys. wymazówek bez podłoża. Tak że dostęp do testów jest zabezpieczony, natomiast decyzje są podejmowanie zgodnie z obowiązującym standardem i w taki sposób są realizowane.

Konsultanci krajowi i główny inspektor sanitarny wprowadzają modyfikacje, różnego rodzaju modyfikacje aktualnie obowiązujących procedur, standardów czy zaleceń. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek przesłanki, że należy rozszerzyć grupę ludzi podlegających testowaniu, natychmiast minister zdrowia będzie podejmował takie decyzje.

Chcę zapewnić, że każda osoba, która spełnia te przesłanki, ma wykonywane testy, jeżeli wymaga kwarantanny, to jest w kwarantannie, jeżeli wymaga izolacji, przebywa w izolatorium. Zabezpieczone są również, to tak obok tego problemu, hotele dla medyków, czyli dla osób, które nie chcą po zakończeniu pracy, np. w oddziale zakaźnym, wracać do swojego środowiska domowego w obawie przed transmisją wirusa do najbliższych. Zabezpieczamy miejsca hotelowe dla wszystkich pracowników, również tych, którzy aktualnie nie są zarażeni i pracują. Tak że te działania mają służyć maksymalnej ochronie pracowników, zabezpieczyć ich przed transmisją koronawirusa. Będziemy podejmować działania, aby występowały w jak najmniejszym odsetku. Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Katarzyna Lubnauer. Pani Minister! Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że oskarżam was o to, że dokonaliście wszystkich działań za późno, że nie wprowadziliście nowych procedur związanych z koronawirusem, nie zabroniliście lekarzom równoczesnej pracy w kilku ośrodkach, nie przeprowadzaliście testów. Obecnie na 1 mln mieszkańców w Polsce jest 4 tys. testów, w momencie, w którym w tych krajach, w których jest najwięcej testowanych w Unii Europejskiej, jest to 48 tys., a średnio jest to kilkanaście tysięcy testów. Oskarżam was o to, że doprowadziliście do sytuacji, w której nie pozwoliliście stosować tych procedur, które dotychczas obowiązują, szpitalom, bo nie miały sprzętu.

Dziękuję.

Szanowni Państwo! Dzięki tym działaniom, które obecny rząd podjął, mamy taką, a nie inną sytuację epidemiczną w Polsce. I naprawdę trzeba dużo złej woli, żeby nie zauważyć, że u nas epidemia rozwija się wolniej niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Te działania, które zostały podjęte przez obecny rząd, spowodowały, że nie mamy takiego dramatu, że nasi pracownicy ochrony zdrowia na szczęście nie stają przed dylematem, kogo podłączyć do respiratora. Zadbaliśmy o to, żeby była odpowiednia liczba miejsc intensywnej terapii w naszym kraju, zadbaliśmy o to, żeby te miejsca były wyposażone. Dbamy o to, aby pracownicy byli chronieni, aby mieli przygotowane standardy, byli odpowiednio wyszkoleni. Gdybyście państwo zadbali kilka lat temu o to, żeby zwiększyć liczbę szkół kształcących lekarzy i pielęgniarki, dzisiaj mielibyśmy o wiele, wiele mniej problemów w tym zakresie.

Bardzo dziękuję, pani minister. Bardzo proszę państwa z Koalicji Obywatelskiej o opuszczenie sali i dostosowanie się do limitu, który został wspólnie ustalony na posiedzeniu Prezydium Sejmu. Kolejne pytanie posłowie Koalicji Obywatelskiej zadadzą w sprawie skutków obostrzeń gospodarczych wprowadzonych w związku ze zwalczaniem pandemii. Pierwsza pytanie zada pani poseł Paulina Hennig-Kloska, klub Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! 14 marca rząd premiera Morawieckiego podjął decyzję o zawieszeniu działalności pierwszych gałęzi gospodarki w naszym kraju. W dalszej kolejności na czas nieokreślony, bo tak naprawdę do dziś właściciele różnych przedsiębiorstw i firm w Polsce nie wiedzą, jaki będzie ich dalszy los, zawieszono działalność galerii handlowych, kin, teatrów, hoteli, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Problem ogromnego spadku przychodów oczywiście ze względów naturalnych dotknął branżę turystyczną i przewozową. W efekcie zamrożenia gospodarki wiele Polek i Polaków utraciło bardzo często jedyne źródło dochodów swojego gospodarstwa domowego. Podejmując takie kroki, rząd w zasadzie od razu powinien mieć w ręce działania osłonowe, które sprawią, że te firmy przetrwają, że te firmy będą mogły po kryzysie wrócić do normalnej pracy. Takich działań zapewnionych przez rząd od razu nie było. Do dziś w zasadzie tarcza nie jest w całości wdrożona. Dlatego mam pytanie, a w zasadzie parę dokładnych pytań o liczby. Ile firm, licząc od 16 marca do dziś, upadło? Wiemy, że przez ostatnie 3 dni marca było to praktycznie 22 tys.

Proszę o podanie dokładnej liczby do dnia przedwczorajszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pan Marek Niedużak. Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

Jest też kilka kwestii, które w pierwszej części pytania miały charakter bardziej ogólny. Jest oczywiste, że ograniczenia, które zostały wprowadzone, muszą być wprowadzane jako reakcja na bardzo dynamiczną sytuację. Chyba pan minister Szumowski bardzo dobrze tę myśl kiedyś wyraził, mówiąc, że on się nie podejmuje robić predykcji na czas dłuższy niż 2 tygodnie w takiej sytuacji. W tak dynamicznej i trudnej sytuacji wszyscy działamy. Tak samo zresztą działają ekonomiści czy analitycy gospodarczy. Właściwie jedyne podejście w tej sytuacji, jakie jest możliwe, to podejście scenariuszowe, z założeniem, że nie mamy jednego planu np. na odmrożenie gospodarki, a szczególnie nie mogliśmy go mieć, nie wiem, miesiąc temu. Możliwe jest tylko i wyłącznie przygotowywanie się na różne scenariusze zależnie od przebiegu epidemii i zależnie od tego, jak długo niezbędne będą surowe, tu chyba wszyscy się zgadzamy, obostrzenia.

Mówię to jako minister właściwy do spraw gospodarki. Po prostu zdaję sobie sprawę, że to nie ministerstwo właściwe do spraw gospodarki powinno grać w tym momencie pierwsze skrzypce.

Tytułem porównania pakiet fiskalny w kryzysie roku 2009 stanowił ok. 1% PKB.

Jeśli chodzi o pomoc nie de minimis, tylko dla dużych firm, to mamy 96% limitu portfela gwarancji wyczerpanego na dzień dzisiejszy.

Widzę licznik, a chciałbym jeszcze mówić o zwolnieniach grupowych. Jeśli chodzi o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego, mamy na wczoraj wieczorem 565 109 takich wniosków. Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 144 964.

Kwestia zwolnień grupowych.

Jeśli chodzi o dane dotyczące nie zgłoszeń, tylko samych zwolnień, to one kształtują się nieco inaczej.

Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Dariusz Rosati, również klub Koalicji Obywatelskiej. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Panie ministrze, myślę, że pan albo jest wprowadzany w błąd, albo pan żyje w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Chcę panu powiedzieć, że skala rzeczywistego zasilenia zapowiedzianego przez rząd, niewypłaconego, wynosi 2,5% PKB.

Proszę nie wprowadzać nas wszystkich w błąd. Reszta to są instrumenty kredytowe związane z uruchomieniem rezerw przez NBP itd. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Według wszystkich prognoz, panie ministrze, gospodarka polska w II kwartale skurczy się o 10%, jak dobrze pójdzie, i w III kwartale - o 5%. Mam pytanie do pana i do rządu:

Dziękuję bardzo. Pani minister Marlena Maląg.

Szanowni Państwo! My to realizujemy. Dane, o których pan minister powiedział, jak najbardziej pokazują środki, bo za tymi liczbami złożonych wniosków stoją konkretne przekazane pieniądze, zarówno z Funduszu Pracy, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i przez nas, co realizujemy poprzez powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy.

Środki te są wypłacane systematycznie. One w żaden sposób nie leżą. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych również zostały dokonane wypłaty, konkretne już wypłaty - na ponad 381 513 tys. zł. I te wypłaty są systematycznie realizowane - dla ochrony ponad 420 tys. miejsc pracy. Tylko w dniu wczorajszym.

Każdego dnia zbieramy te informacje - one będą za chwilę dostępne też na licznikach w powiatowych urzędach pracy, w wojewódzkich urzędach pracy i na naszej stronie. Po to, abyście państwo mieli wgląd do tego, że składane wnioski - bo za nimi jest konkretny pracodawca, konkretny pracownik, konkretna rodzina - są nie tylko zbierane sprawnie, bo są zbierane sprawnie, ale są także realizowane wypłaty, bo to jest naszym celem. Bardzo dziękuję, pani minister. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zadają pytanie w sprawie działań, jakie podjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z trudną sytuacją artystów. Bardzo proszę. Pierwsze pytanie zadaje pani poseł Joanna Lichocka. Bardzo mi przykro. I proszę nie podnosić głosu tutaj, na sali. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Epidemia uderzyła w świat ludzi kultury bardzo mocno. Nie działają teatry, nie produkuje się filmów, nie produkuje się seriali, nie ma wystaw, nie ma nowych wydarzeń artystycznych. Bardzo często ich twórcy mają z dnia na dzień bardzo ograniczone źródła dochodu. To nie są pracownicy na etatach, z gwarancją określonej pensji.

Dziękuję. Bardzo dziękuję. Odpowiada wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego pan wicepremier Piotr Gliński. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ono jest ważne, bo faktycznie może róże nie są najważniejsze, gdy płoną lasy, ale te róże, jak państwo wiecie, wszystkim nam są potrzebne, także tym, którzy na pierwszej linii gaszą pożary lasów. Dlatego niezwłocznie po ogłoszeniu pierwszych ograniczeń związanych z epidemią przystąpiliśmy do prac nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności sektora kultury.

Myśmy przyjęli na współprowadzenie i powołali wiele nowych instytucji prowadzonych przez ministerstwo kultury, to ponad 60 nowych podmiotów działających w kulturze, a więc także takich podmiotów, gdzie ludzie mają etaty, gdzie mają stabilną pracę. Drugim takim systemowym działaniem była walka ze śmieciówkami.

To jest specyfika tego sektora i ludzie kultury w dużej mierze na to się godzili. Ona została zatrzymana niestety przez ostatnie 2 miesiące, gdy doszło do przestawienia naszych działań na inny kierunek, ale toczą się prace nad ustawą systemowo regulującą status artysty w Polsce, wraz z powołaniem funduszu ubezpieczeń. Nie było cywilizowanego rozwiązania w sferze zabezpieczenia potrzeb artystów i ludzi kultury. Ci ludzie w dużej mierze nie mieli cywilizowanego zabezpieczenia, jeśli chodzi o kwestię ubezpieczeń. Myśmy to stworzyli, ta ustawa jest praktycznie gotowa. Ona przez 2 lata była przygotowywana w debacie, w dyskusji z całym środowiskiem kultury.

To wszystko dotyczy także ludzi kultury. Ja już nie jako minister kultury, ale jako przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego odpowiadam za kwestię organizacji pozarządowych. Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem w tej kwestii, zadbał o to, żeby w obu tarczach były także poruszane i zapewnione sprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych, ponieważ wiele działań kulturalnych jest realizowanych w formie prawnej organizacji pozarządowych i te sprawy zostały także ujęte. Organizacje pozarządowe w dużej mierze zostały zrównane z przedsiębiorstwami. Wielkim, myślę, istotnym zabezpieczeniem ludzi kultury jest postojowe, związane z sytuacją osób, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne, zlecenia, o dzieło, a także samozatrudnionych. Jak państwo wiecie, postojowe zostało przedłużone do 3 miesięcy, a więc to zabezpieczenie podstawowe w wysokości 80% płacy minimalnej dla tych osób, które utrzymywały się z pracy w tej formie, jest zapewnione. Jak powiedziałem, także organizacje pozarządowe zostały zrównane i to też wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi kultury. Przede wszystkim to jest program „Kultura w sieci”, który w tej chwili już ruszył. Wnioski są zbierane do 20 kwietnia. Ten program jest podzielony na osoby fizyczne i na podmioty, nie będę wchodził w szczegóły. To jest w tej chwili w pierwszym rzucie 20 mln zł. My mówimy o tym, że to jest pierwszy rzut. Jeżeli będzie za mało, będziemy starać się dosypać do tego. Zwiększyliśmy także programy ministerstwa. Minister ma 32 programy. O 60 mln w ostatnim miesiącu zwiększyliśmy te programy, w postaci odwołań, żeby można było jeszcze zasilić sektor. To dotyczy i zabytków, i koncertów muzycznych, które są oczywiście przesuwane na jesień czy na późniejszy termin, i wielu innych działań w obszarze kultury. Planujemy także dodatkowy program po epidemii, niestety nie wiemy, kiedy to będzie. Oprócz tego w ministerstwie funkcjonuje Fundusz Promocji Kultury, którego część jest przeznaczana na zapomogi socjalne dla twórców i artystów. Myśmy natychmiast zwiększyli pulę tego funduszu, on już jest wypłacany. Te osoby mają już w tej chwili wypłacane zapomogi. Następna komisja będzie jeszcze w tym tygodniu. My je wszystkie w ciągu najbliższych dni rozpatrzymy i ta bezpośrednia, podstawowa pomoc zostanie przekazana.

To jest 500 mln zł dla ludzi z sektorów kreatywnych. Mogą oni korzystać z tego rodzaju dogodnych pożyczek, kredytów, wsparcia w ramach tego programu.

To są kwestie, w które nie chcę wchodzić szczegółowo, bo one są bardziej profesjonalne, natomiast one umożliwiają funkcjonowanie kultury w obecnej sytuacji w sieci i ułatwiają funkcjonowanie producentów filmowych, ludzi kina, ludzi filmu. Tak więc branża kultury, obok branży hotelowej, restauracyjnej, turystycznej, została specjalnie włączona w pierwszej tarczy kryzysowej jako ta, która może wystawiać vouchery, czyli przenosić swoje zobowiązania aktualne na przyszłość.

Następne są przygotowywane, ale dopóki nie zostaną przyjęte przez Sejm - mówię o trzeciej tarczy antykryzysowej - to może nie ma sensu, żeby o nich w tej chwili mówić.

A więc uelastycznienie, przeniesienie terminów, a także przeniesienie terminów dotyczących zobowiązań podatkowych, zobowiązań sprawozdawczych - to wszystko zostało wprowadzone praktycznie w ciągu jednego miesiąca dla polskiej kultury. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa szkół pożarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, o której przedstawienie wnosił Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Czy jest na sali pan poseł Wiesław Szczepański, który jest przedstawicielem.

Nie wiem, czy to jest dobre określenie.

Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Wiesława Szczepańskiego. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W Polsce funkcjonuje kilka szkół pożarniczych: podoficerska w Bydgoszczy, aspirantów w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie oraz ta najważniejsza - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie szkoląca oficerów służby pożarniczej. Szkoły te szkolą elity polskich strażaków. Tak jak oni czuwają nad naszym dobytkiem i zdrowiem, tak i państwo, które ich kształci, winno zapewnić im bezpieczeństwo i zdrowie. Ostatnie dni pokazały niestety, że tak nie jest.

Istnieje podejrzenie, że jest tam również osoba zakażona. Mimo że od 16 kwietnia zamknięte zostały cywilne szkoły i uczelnie, w SGSP i innych szkołach pożarniczych nadal trwały zajęcia, a studenci nadal byli skoszarowani w dużej grupie. Stwarzało to zagrożenie, możliwość potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem. Nie są to wszystkie osoby, które mogą być zarażone. Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA, która decyzją rządzących już niedługo zostanie zlikwidowana, podjęła decyzję o kwarantannie dla podchorążych wszystkich kompanii tej jednostki, a więc ponad 300 osób. Pracowników cywilnych uczelni wysłano do domu bez jakichkolwiek badań. O zagrożeniu życia i zdrowia podchorążych media informowały w serii artykułów już od wielu dni. Pierwsze objawy u podchorążych wskazujące na zarażenie pojawiły się u niektórych już 6 kwietnia. Kierownictwo jednostki oskarżało podchorążych o symulanctwo. Testy na obecność koronawirusa przeprowadzono w szkole dopiero w dniach 11 i 12 kwietnia. W tym czasie podchorążowie wychodzili swobodnie na miasto, wiele razy, według informacji mieszkańców, grupowo, stanowiąc potencjalnie zagrożenie dla innych osób. Wychodzili również poza obręb uczelni, bo nadpowietrzne przejście nad ulicą między budynkami uczelni od wieków jest nienaprawione. Kierownictwo szkoły wykazało się w tym okresie rażącą niekompetencją zawodową i dowódczą oraz brakiem jakichkolwiek zasad etyki i moralności, co naszym zdaniem odbiera im możliwość pełnienia funkcji dowódczych uczelni kształcącej kadrę dowódczą polskiego pożarnictwa. W szkole panował chaos. Według doniesień mediów, z informacji uzyskanych od podchorążych, osoby zdrowe dostawały rozkaz noszenia posiłków chorym kolegom bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Brak było w pewnych okresach środków dezynfekujących. Informowano, co wywołuje zażenowanie, że dowództwo uciekło do domu. Każda sprawa, którą zgłaszali podchorążowie, załatwiana była dopiero po nagłośnieniu medialnym. Kierownictwo szkoły wykazało kompletną indolencję, brak umiejętności zarządzania w kryzysie, co stworzyło warunki do dalszego wzrostu liczby chorych. Interwencja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a więc ubezwłasnowolnienie władz szkoły pożarnictwa i przejęcie ich roli w zarządzaniu kryzysowym, spowodowała podjęcie działań zaradczych i ratowniczych wobec osób zakażonych i tych, w przypadku których możliwe jest zakażenie. Pytam, dlaczego trwało to tak długo, zanim zareagował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Może dlatego, że w tym czasie jeździł po Polsce i wymieniał swoich na swoich: pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Opóźnienia działań mających na celu opanowanie zagrożenia spowodowały świadome narażenie dużej grupy studentów na utratę zdrowia, a nawet życia. COVID-19 pozostawia trwałe zmiany w organizmie zarówno u osób, które chorowały na koronawirusa, jak i u tych, które przeszły zarażenie bezobjawowo. Może to w przyszłości wyeliminować tych młodych ludzi ze służby, a więc stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych od uczelni. Rodzice oddali tych młodych ludzi pod opiekę państwa, ale państwo zawiodło. Czy ono wystarczy?

Ale czy tylko on jest winien? Czy nie jest winne całe kierownictwo szkoły? Kępka jest autorem książki „Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej” Niestety wiedzy tej nie wykorzystał w zarządzanej przez siebie uczelni. W normalnym świecie, gdyby był człowiekiem honoru, sam podałby się do dymisji, a nie wnioskował o odwołanie zastępcy. Panie Ministrze! Jak wygląda sytuacja i zabezpieczenie przed koronawirusem w innych szkołach pożarniczych w Polsce? Kto poniesie odpowiedzialność zawodową, finansową, polityczną, a nawet karną za powstałe zaniedbania? Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o udzielenie odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od 12 marca zawieszone są zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Mimo zawieszenia zajęć dydaktycznych studenci podchorąży pozostali w szkole głównej straży pożarnej i innych szkołach pożarniczych, ponieważ te placówki posiadają swoje jednostki ratowniczo-gaśnicze z wyznaczonymi rejonami chronionymi. Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest jednostką organizacyjną PSP i musi utrzymywać odpowiedni potencjał ratowniczy na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na swoim terenie. W tym wypadku chodzi o dzielnicę Żoliborz w Warszawie. Dodatkowo szkoły wchodzą w skład centralnego odwodu operacyjnego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na odwód operacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego składa się 80 podchorążych szkoły głównej straży pożarnej i po 50 studentów pozostałych uczelni. Biorąc pod uwagę charakter tej służby i system 24 godziny na 48 godzin, dla potrzeb operacyjnych musi być skoszarowanych ok. 300 podchorążych szkoły głównej straży pożarnej. Jeżeli chodzi o wydarzenia, jakie miały miejsce w tej szkole, to pierwsze informacje o studentach skarżących się na objawy podobne do tych w przypadku COVID-19, czyli brak smaku, węchu, podwyższona temperatura, miały miejsce 5 kwietnia w niedzielę. 7 kwietnia we wtorek pojawiły się pierwsze artykuły medialne opisujące tę sprawę. 10 kwietnia w piątek przeprowadzono pierwsze testy na obecność koronawirusa.

Wirus został stwierdzony u 47 podchorążych. 15 kwietnia w powtórnym badaniu dodatnie wyniki stwierdzono u 4 kolejnych podchorążych. Łącznie dodatni wynik badania stwierdzono u 51 podchorążych.

Studenci nie są hospitalizowani, bo mają na szczęście łagodne objawy koronawirusa. W uzgodnieniu ze służbami sanitarnymi podjęto decyzję o podzieleniu podchorążych objętych kwarantanną na mniejsze grupy. Pozostali odbywają ją w centralnej szkole służby pożarniczej w Częstochowie, w szkole aspirantów PSP w Bydgoszczy i w wojewódzkich ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Tylnej Górze, Pionkach i Olsztynie. Kwarantanna prowadzona w kilku lokalizacjach pozwala ograniczać potencjalne zakażenia do mniejszej grupy i zapewnia podchorążym dobre warunki bytowe na czas trwania kwarantanny. Przewóz podchorążych realizowany był w oparciu o środki transportu PSP.

Miedzy 7. a 9. dniem kwarantanny, zgodnie z decyzją służb sanitarnych, zostaną przeprowadzone kolejne testy u podchorążych. Przed dyslokacją podchorążowie przebywali na terenie szkoły głównej straży pożarnej. W pomieszczeniach szkoły specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna Warszawa 6 prowadziła fumigację, czyli gazową dezynfekcję pomieszczeń, która jest najbardziej skuteczna. Podchorążowie przebywali w tym czasie m.in. w salach i na korytarzach szkoły. Wysoka Izbo! W opinii komendanta głównego państwowej straży pożarnej (Dzwonek), którą podzielam, doszło do zaniedbania, bardzo poważnego zaniedbania. W tym momencie komendant główny straży pożarnej skierował wniosek o odwołanie prorektora, zastępcy komendanta szkoły głównej straży pożarnej do spraw operacyjnych, starszego brygadiera Jarosława Zarzyckiego.

Prorektor miał też wprowadzać w błąd bezpośrednich przełożonych, sugerując, że podchorążowie mogą symulować chorobę, licząc na możliwość wyjazdu do domu na święta. 15 kwietnia komendant główny państwowej straży pożarnej powołał specjalny zespół do spraw wyjaśnienia przyczyn zdarzeń w szkole głównej straży pożarnej. Zespół ma ustalić przyczynę transmisji wirusa do szkoły w sytuacji, gdy skoszarowani w niej studenci podchorążowie nie wychodzili poza jej teren, i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zawiodły procedury, kto za to odpowiada i jak tego typu sytuacji ustrzec się w przyszłości. Jeżeli chodzi o sytuację w pozostałych szkołach, to nie ma sygnałów o jakichkolwiek zagrożeniach, natomiast służby po tych wydarzeniach warszawskich są bardzo wyczulone i jeżeli pojawią się jakiekolwiek sygnały ze strony studentów, na pewno będą one błyskawicznie weryfikowane. Doszło do sytuacji niedopuszczalnej, gdzie nie okazano szacunku i zaufania podchorążym i studentom, stąd też pierwsze konsekwencje zawodowe. Prorektor, który za to odpowiadał, który wprowadzał swoich przełożonych w błąd, który przez kilka dni sugerował, że mamy do czynienia z symulantami, którzy chcieli wyjechać do rodzin na święta, poniósł konsekwencje. Komisja rozpoczęła działania, a sprawa będzie wnikliwie zbadana. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Informuję, że zgłosili się posłowie do dyskusji. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? Jeżeli nie, to zamykam listę mówców. Otwieram dyskusję.

W takim razie proszę o zabranie głosu pana posła Bartłomieja Sienkiewicza, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Skąd pan bierze takie kadry? Skąd pan bierze kadry w ministerstwie, które porzucają swoich kadetów, które narażają ich na chorobę? Jak to jest możliwe, że w służbie państwowej doszło do tak dramatycznego nadużycia? Skąd oni są? Oni są z pana nominacji. To są pańscy ludzie, to są pańscy ludzie po wymianie kadrowej w MSW od szczebla generałów do szczebla najniższego. To nie jest przypadek. Jeśli dzisiaj o tym mówimy, to dlatego, że szkoła główna pożarnictwa w Warszawie jest symbolem tego, co dzieje się w Polsce w trakcie koronawirusa: niekompetencji, opóźnienia, lekceważenia problemu, a potem - czego? - hucpy, po prostu wielkiej hucpy, bo prawdę mówiąc, z trudem odczytane przygotowane przemówienie, które przed chwilą usłyszeliśmy z ust pana ministra, nic nie wyjaśnia, nie wyjaśnia ani jednego zarzutu, który został tutaj przed chwilą postawiony.

A na samym końcu okazuje się, że mamy jeden z najwyższych wskaźników zakażeń służby medycznej, mimo że jesteśmy jeszcze przed szczytem pandemii. Tak naprawdę Polska dzisiaj to jest właśnie Szkoła Główna Służby Pożarniczej. To jest reguła, to nie jest wyjątek. Jeśli chcecie dzisiaj urządzać kolejne propagandowe wydarzenia z największym samolotem na świecie, z opowieścią pana premiera, że jesteśmy najlepsi i inni na nas się wzorują, to są to - tak - właśnie te próby zakłamania rzeczywistości. A rzeczywistość w Polsce podczas pandemii to jest szkoła (Dzwonek), którą pan nadzoruje. Proszę o zabranie głosu panią poseł Katarzynę Kretkowską, Lewica. Wysoka Izbo! Przed chwilą pan minister powiedział, że wszyscy podchorąży tej szkoły zostali przetestowani, ale nie powiedział, kiedy zostali przetestowani. Nie powiedział pan, że zostali przetestowani o wiele, wiele za późno, po tym jak już zdążyli krążyć po Polsce, krążyć po jednostkach, po własnych domach, po Warszawie, zarażając inne osoby. W materiale przedstawionym przez TVN24 rzecznik komendy głównej szkoły pożarnictwa poinformował, iż każdy pracownik szkoły miał dostęp do testów oraz że była to powszechnie znana informacja i każdy mógł zgłosić się w sobotę i niedzielę na testy. Proszę zatem o odpowiedź na piśmie, kto, kiedy i w jaki sposób poinformował o tym fakcie wszystkich pracowników i funkcjonariuszy szkoły. Po drugie, proszę odpowiedzieć na piśmie, czy zespół powołany do wyjaśnienia całej tej sytuacji zamierza prowadzić rozmowy tylko z kierownictwem, czy też z pozostałą społecznością szkoły, bo tak naprawdę opinia publiczna dowiedziała się o tej sytuacji z desperackich apeli w mediach społecznościowych samych podchorążych. Dlaczego kierownictwo szkoły nalegało, żeby podchorążowie pełnili służbę w jednostce, kiedy było już wiadomo, że występują u nich symptomy zarażenia? Czy odwołany komendant, zastępca komendanta, prorektor Jarosław Zarzycki jest obecnie w dyspozycji komendy głównej, czy też już ma złożony raport o zaopatrzenie emerytalne z datą wsteczną? Jak wytłumaczyć fakt, że pomimo obowiązujących procedur dowódca jednostki i zastępca komendanta chcieli, ażeby podejrzany o zakażenie, o zarażenie wirusem podchorąży jechał do szpitala zakaźnego autobusem wraz z innymi osobami? Dlaczego strażacy z jednostki, którzy od 10 kwietnia przebywali w domach, nie zostali skierowani na badania? Obecnie (Dzwonek) większość z nich przebywa na kwarantannach. I wreszcie, ile jest w Polsce podobnych szkół i uczelni mundurowych, w których studenci pozostają skoszarowani, nie są testowani, w których nie zostały wdrożone obowiązujące w Polsce nakazy, zakazy i procedury służące walce z epidemią? Odpowiedź na to pytanie nie została udzielona przez pana ministra. Wypowiedź była enigmatyczna. Proszę odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Zanim zacznę, zanim zadam pytanie, szanowni państwo, pozwólcie, że jednak mimo wszystko podziękuję z tej mównicy strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, jak również z ochotniczej straży pożarnej za to, co robią dzisiaj, każdego dnia i często być może z narażeniem swojego życia. Bo wydaje mi się, panie ministrze, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie w środki ochrony osobistej właśnie strażaków, to na panu spoczywa wielki obowiązek zadbania o to. Oni są też na pierwszej linii frontu. Bardzo proszę, panie ministrze, żeby pan o tym pomyślał. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, szanowni państwo, to mam konkretne pytania.

Chciałbym, żebyśmy się tutaj, szanowni państwo, tego dowiedzieli. Bardzo bym prosił, żeby ta sytuacja była cały czas monitorowana i żebyśmy na bieżąco tę informację otrzymywali. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Dariusza Jońskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kilka dni temu lekarze i pielęgniarki pytali nas i prosili o wsparcie, i proszą dalej o wsparcie, dlatego że brakuje masek, brakuje środków ochrony osobistej.

Jest kompletny chaos. Otóż ci, którzy na co dzień niosą pomoc - to dotyczy pielęgniarek, lekarzy czy strażaków - dzisiaj sami proszą nas o pomoc, m.in. dlatego, że nie potraficie sobie państwo poradzić i pomóc im w trudnej sytuacji. Ale to, z czym mamy do czynienia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, to jest już niekompetencja, chaos i w tej sprawie żądamy konkretnych postępowań dyscyplinarnych. Otóż po zgłoszeniach jednej z grup, która jako pierwsza wskazywała najwięcej zarażeń, usłyszeli oni od zastępcy komendanta do spraw operacyjnych, że symulują. Otóż jeśli tak jest, że kierownictwo szkoły głównej pożarnictwa uważa, że mundurowi studenci symulują - mało tego, oni nazwali ich nawet nierobami za to, że nie chcieli prowadzić zajęć podczas zakazu nałożonego przez komendę główną - to chciałbym zapytać pana ministra, dlaczego nie został odwołany w tej sprawie sam komendant, dlaczego w tej sprawie nie ma postępowań dyscyplinarnych. Na ostatnie wyniki ma czekać 12 osób. Dlaczego to tak długo trwa i kiedy to się skończy? Dziękuję. Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Studenci Państwowej Straży Pożarnej są studentami mundurowymi. To się wiąże z tym, że mają inne obowiązki aniżeli pozostali studenci. Muszą często przebywać w grupach, nie mogą pracować tylko zdalnie. Czy po tych przykrych doświadczeniach wprowadzono pewne zmiany proceduralne, organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo studentów również w innych szkołach mundurowych? Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz głos zabierze pani poseł Monika Pawłowska, Lewica.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szkoła Główna Służby Pożarniczej to chluba straży pożarnej w Polsce. Służby codziennie narażają swoje zdrowie i życie, codziennie dają nam przykład do naśladowania, aby nie poddawać się w codziennej walce z koronawirusem. Pytamy ministra spraw wewnętrznych i administracji: Jak można dopuścić do tego, że umyślnie narażacie państwo zdrowie i życie strażaków i pracowników uczelni na niebezpieczeństwo? Jak można dopuścić do tego, że dowództwo zarówno jednostki ratownictwa gaśniczego, jak i uczelni nie podjęło na czas żadnych kluczowych decyzji w czasie trwania pandemii? Czy gorączka, brak smaku, węchu, złe samopoczucie to mogą być objawy koronawirusa, czy nie? To są pytania do ministra, bo ministerstwo nie wie, że szkoła powinna być zamknięta już dawno temu. Ministerstwo nie wie, że studenci choćby z podejrzeniem powinni być odizolowani, a pozostali powinni być pod stałą kontrolą. Ministerstwo nie wie, że nic nie wie. A więc co wie ministerstwo, skoro ministrem jest jednocześnie minister koordynator służb specjalnych? Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu panią poseł Ewę Szymańską, Prawo i Sprawiedliwość. W takim razie, skoro pani poseł jest nieobecna, proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Borysa, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ta sytuacja jest sytuacją podwójnie złą i trudną, dlatego że wydarzyła się w przestrzeni Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, tej, która przecież kształci oficerów, elitę służby, która ma przecież w Polsce najwyższe zaufanie, ludzi, którzy w całej Polsce swoją odwagą, profesjonalizmem ratują życie i zdrowie Polaków. Dlatego tym bardziej ten przykład musi być wyjaśniony, jeżeli zostały złamane podstawowe elementy związane z procedurami, bezpieczeństwem, a przede wszystkim prawdą. Bo taka sytuacja może zdarzyć się wszędzie, zdarza się w szpitalach, ale istotą służb jest wyjaśnienie prawdy i szybkie zadziałanie zgodnie z procedurami, to jest wymóg polskiego oficera. Dlatego zadaję pytanie, będąc informowany przez pracownika czy pracowników tej szkoły: Czy to nie jest tak, że cały system odpowiedzialności jednak powinien być skupiony na władzach uczelni, które po prostu zaniedbały tę sprawę czy też ukrywały fakt zarażenia pracowników? Czy nie jest tak, że pan rektor prof. Paweł Kępka jednak otrzymał ten awans za państwa rządów?

Normalnie takie awanse trwają latami. Chciałbym o to zapytać, będąc poinformowany przez profesorów tej uczelni, dlatego że odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, [[Dzwonek]] spada także na pana rektora i z tego należy wyciągnąć daleko idące konsekwencje na przyszłość, żeby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zadanie pytania, o zabranie głosu pana posła Pawła Krutula, Lewica. Panie Ministrze! Panowie Strażacy! Posłowie, Posłanki! Jako członek zespołu strażaków IX kadencji Sejmu chciałbym zadać następujące pytania: Czemu mimo ujawnienia objawów u 16 podchorążych nie wstrzymano ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez dział szkolenia poligonowego? Czemu po ujawnieniu objawów u 16 podchorążych zwiększono wymiar zajęć praktycznych na poligonie w Nowym Dworze Mazowieckim? Czy wszyscy funkcjonariusze prowadzący ćwiczenia zostali przebadani testem na obecność koronawirusa? Jeśli nie, czy i kiedy zostaną przebadani na tę okoliczność? Kto był odpowiedzialny za zakwalifikowanie funkcjonariuszy potencjalnie poddanych ekspozycji na przeprowadzanie tych testów? Kiedy nastąpiło powiadomienie o trwaniu testów, w jaki sposób i komu przekazano taką informację i na czyje polecenie? Proszę o odpowiedź na te pytania na piśmie. A wszystkim strażakom chcę podziękować, że stoją na pierwszej linii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu panią poseł Ewę Szymańską, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To, co się wydarzyło, to już się wydarzyło i już się nie odwróci. Mam pytanie: Jak sobie radzą inne szkoły pożarnictwa i nie tylko szkoły pożarnictwa, ale też szkoły policyjne, tam gdzie są duże skupiska ludzi? Jak wygląda sprawa w szkole pożarnictwa, o której mówimy?

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Waldemara Andzela.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym podziękować jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale także wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, za działania, które podejmują na co dzień Państwowa Straż Pożarna oraz druhowie z ochotniczej straży pożarnej, którzy są na pierwszej linii w walce z koronawirusem. Chciałbym spytać pana ministra, aby pan minister powiedział, jakie działania podejmują Państwowa Straż Pożarna, ochotnicza straż pożarna oraz pozostałe służby mundurowe w walce z koronawirusem. Jeszcze raz, tak jak mówię, chciałbym podziękować. Mam pełne zaufanie do tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, a także pan minister i podległe mu służby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W szkole głównej straży pożarnej zostały wprowadzone pokoje dwuosobowe. Osoby przebywające tam miały się wymieszać między sobą, mimo że nie znały wyników swoich testów na COVID-19. Rektor groził studentom konsekwencjami dyscyplinarnymi za wypowiedzi w mediach społecznościowych. Konkretnie straszył studentów, że napisze wnioski o wstrzymanie nadania pierwszego stopnia oficerskiego tym, którzy będą opisywać sytuację, jaka ma miejsce w szkole. W ilu jeszcze szkołach, akademikach, komendach Policji i straży pożarnej jest podobnie? To wierzchołek góry lodowej. Dlaczego rząd godzi się na cenzurę służb mundurowych? Dlaczego państwo nie chroni tych, co walczą o nasze życie i zdrowie? Dlaczego zamiast pomocy Polki i Polacy otrzymują koleje represje i chaos? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Małgorzatę Prokop-Paczkowską, Lewica. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówił pan do nas tak cicho. Nie wiem, czy nie zjadł pan dzisiaj śniadania, czy jest panu po prostu wstyd i nie mógł pan wydobyć z siebie głosu. A teraz pytania. Proszę o odpowiedź na piśmie. Czy dowódcy kompanii, lekarz szkolny, prorektor znali procedury przeciwdziałania epidemii? Czy został powołany stosowny sztab kryzysowy? Dlaczego temperaturę mierzono pirometrem? Czy miał wykonany test? Czy komendant rektor był na bieżąco informowany o sytuacji? Dlaczego nie zaniechano ćwiczeń na boisku, na siłowni i na wspinalni? Jakie środki ochrony indywidualnej zostały przekazane funkcjonariuszom? Dlaczego czynne były aż cztery bramy i dwa biura przepustek? Dlaczego nie zamknięto kładki między obiektami, aby ograniczyć przemieszczanie się wewnątrz szkoły? Czy podchorążowie byli wożeni na badania okresowe autobusem? Którzy dowódcy pracowali zdalnie? Czy były takie sytuacje, że żadnego z dowódców nie było w danych kompaniach?

I obietnica: nie zostawimy was z waszymi problemami. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią poseł Martę Wcisło, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jesteśmy przygotowani do walki z koronawirusem, wyprzedzamy Europę - zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Czy jesteśmy przygotowani? Jak to się ma do sytuacji w szkole wyższej służb pożarniczych, gdzie panuje chaos, jak informują sami podchorążowie, gdzie osoby, które jeszcze do niedawna nie były chore, po 2 dniach mają pozytywne testy, a osoby, u których wykryto COVID-19, są w prowizorycznych izolatkach, w których nie mają dostępu do prysznica, w których brakuje węzłów sanitarnych? Osoby, co do których nie podjęto jeszcze decyzji, koczują na korytarzach, śpią na stołach, krzesłach. Tak wygląda sytuacja w szkole służb mundurowych. Kto za to odpowiada? Kto odpowiada za ten chaos? Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby studenci, żeby podchorążowie nie musieli szukać pomocy w mediach i w Internecie, żeby mogli normalnie wrócić do domu bądź być poddani przyzwoitej kwarantannie, żeby byli wyposażeni w środki ochrony osobistej, żeby zadbano o ich zdrowie? To są osoby, które w przyszłości będą ochraniać, będą udzielać pomocy. Kto nadzoruje szkołę wyższą? Kto za to odpowiada? Bo to jest wstyd i hańba. Gdzie są procedury? Szkoła, która powinna stosować się do wszystkich regulaminów, łamie wszystkie zasady. Panie Marszałku! Proszę o odpowiedź na pytanie: Kto odpowiada za chaos w szkole głównej pożarniczej? Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę o zabranie głosu pana posła Rafała Adamczyka, Lewica. Jeżeli posła nie ma, to pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Też nie widzę.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W mediach krążą nagrania pokazujące leżących na korytarzach, na podłodze, na ławkach studentów.

Jednym słowem: skandal. Skandal i wielki chaos, panie ministrze.

Według studentów dla dowództwa najważniejsze jest teraz sprzątanie terenu szkoły. Chciałabym, żeby pan się do tego ustosunkował. Jesteśmy świadkami przede wszystkim rażącej niekompetencji: niekompetencji zawodowej i niekompetencji dowódczej. Konsekwencje do dzisiaj nie zostały wyciągnięte, bo to pan, panie ministrze, odpowiada za to, co tam się wydarzyło. To pan, panie ministrze Kamiński, powinien podać się do dymisji, a jeśli nie ma pan na tyle odwagi, jeśli nie ma pan na tyle honoru, to powinien to zrobić pan premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Szczerbę, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ilu tragedii można by było uniknąć, gdyby od samego początku były przeprowadzane testy? To nie jest obowiązek rektora - przeprowadzanie testów i wykrywanie wirusa. Ile jest miejsc w Polsce, gdzie groźba zakażenia jest przedmiotem czyjejś opinii, a nie procedur medycznych? Jakie procedury, panie ministrze, są w innych szkołach, także panu podległych, np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie? Dzisiaj mogliby służyć społeczeństwu, mogliby pomagać w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, oddziałach medycyny paliatywnej. Taka sama sytuacja, Wysoka Izbo, jest w Wojskowej Akademii Technicznej: 350 podchorążych i czterech żołnierzy WAT jest w kwarantannie, u 11 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. Czy istnieją procedury - w sytuacji kiedy pojawia się podejrzenie, a mamy do czynienia ze zbiorowością, która zazwyczaj jest skoszarowana, mieszka w domu studenckim - dotyczące szybkiego działania? To jest konkretna sprawa. Nie może być takich sytuacji. To, co wyrabia pan wojewoda Radziwiłł, to jest niebywały skandal. Jest ustawa dotycząca zakażeń, jest ustawa, która mówi o tym, jakim osobom nie można dać nakazu pracy, ponieważ podlegają wykluczeniu. Są to, panie ministrze, osoby powyżej 60. roku życia, są to osoby opiekujące się małoletnimi dziećmi. Pan wojewoda Radziwiłł takim osobom daje nakazy pracy, a następnie karze je finansowo. Ten przypadek matki karmiącej 5-miesięczne dziecko jest przypadkiem niebywałym i apeluję do pana, żeby pan tę kwestię zanalizował i wyciągnął konsekwencje wobec wojewody Radziwiłła. Dziękuję bardzo.

Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak podał Onet, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej osobom zarażonym posiłki roznoszą osoby zdrowe, zgodnie z rozkazem dowództwa. Mają to robić bez wystarczającego zabezpieczenia. Studenci tej szkoły, dzwoniąc do oficera dyżurnego w związku z kończącymi się środkami dezynfekującymi, słyszą taką oto odpowiedź, że mają to sobie jakoś załatwić. Panie Ministrze! Czy taka jest polityka rządu? Czy taka jest polityka pańskiego ministerstwa? Koszarujecie ludzi, nakładacie na nich obowiązki, a później mówicie: Niech sami sobie zorganizują ochronę. Przecież to jest niepoważne. Nie wiem, czy pan minister identyfikuje się z takim postępowaniem, ale na pana miejscu po prostu podałbym się do dymisji. To oznacza, że pana ludzie - ci, których pan wybrał, nominował, postawił na stanowisku - nie spełniają najwyższych wymagań, jakie powinni spełniać ludzie, którzy zostali postawieni na tak poważnym stanowisku, w czasie epidemii, czyli w czasie zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Tymczasem działania podejmowane przez pana ludzi - tych, których pan wyznaczył, tych, których pan posłał, żeby kształcili przyszłe kadry służby pożarniczej. Co więcej, jaki przykład ludzie, którzy później mają ratować obywateli w sytuacji różnych zagrożeń, otrzymują od swojego kierownictwa, od kierownictwa, które zostało tam przysłane przez pana ministra? Panie Ministrze! Jeżeli pan może zaprzeczyć, proszę zaprzeczyć. Jeżeli pan potwierdza to, co przytoczył Onet, to, co przed chwilą przeczytałem. W tej sytuacji prawdziwy polityk, który ma na celu dobro państwa, podaje się do dymisji. Panie ministrze, czy pan jest prawdziwym politykiem mającym na celu dobro państwa?

Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Korzystając z tego, że mam okazję zadać panu ministrowi pytanie, chciałam zapytać nieco szerzej.

Dlaczego służb w Polsce nie wyposażono w środki ochrony indywidualnej?

Dziękuję bardzo. Lista osób zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Wiesława Szczepańskiego. Będzie mi się lepiej czytać. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na sztandarach strażaków widnieje napis: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W szkole głównej pożarnictwa panuje obecnie zastraszenie. Rektor grozi dzisiaj studentom konsekwencjami dyscyplinarnymi za wypowiedzi w Internecie i mediach społecznościowych. Czy nie uważa pan, że ta sprawa powinna zostać skierowana do rzecznika praw obywatelskich? Jest to świadome narażanie ich na utratę zdrowia i życia. Według mojego klubu istnieje potrzeba wymiany całej kadry kierowniczej w szkole, nie tylko zastępcy rektora pana bryg. Jarosława Zarzyckiego. Za funkcjonowanie JRG szkoły głównej odpowiadał on, ale po jego odwołaniu te obowiązki pełni bryg. Tomasz Klimczak, który do tej pory jest też dowódcą pododdziałów szkolnych. On również zarzucał studentom symulowanie. Pracownicy uczelni nie mogą zgłosić się w złym stanie zdrowia do sanepidu powiatowego. Słyszą tam: Zgłoszenie nie zostanie nawet zarejestrowane.

Nie wiedzą, czy są chorzy, czy nie zarażają swoich najbliższych. Nikt nie chce im pomóc. Sanepid MSWiA nie odbiera telefonu. Myślę, że powinien pan zrobić z tym porządek. Jak to jest, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej od dziennikarza Onetu dowiedziała się, że jeszcze przedwczoraj 12 studentów nie miało wyników testów? Czy zamierza pan powiadomić prokuraturę? Powinna ona wszcząć śledztwo w sprawie wydarzeń w szkole.

Przyszłych oficerów mają pilnować przyszli chorążowie. Minister spraw wewnętrznych i administracji, realizując dyspozycje wynikające z ustawy, znowelizował 17 lipca 2017 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W § 4 pkt 3 określił, że organizacja funkcjonowania KSRG przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na obszarze kraju obejmuje w szczególności opracowanie zasad postępowania podczas wystąpienia zagrożenia niezidentyfikowaną przesyłką oraz organizacji transportu materiałów biologicznych, a także opracowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. Czy na podstawie obowiązującego rozporządzenia przed pojawieniem się koronawirusa opracowane zostały zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi? Czy zaopatrzono jednostki OSP i PSP w niezbędne środki ochrony osobistej dla strażaków, którzy mogą uczestniczyć w działaniach wspomagających, o których mowa w ustawach? Czy opracowano zasady postępowania w przypadku możliwości wystąpienia zakażeń na dużą skalę w szkole pożarniczej? Czy opracowano zasady współdziałania z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym? Myślę, że dobrze by było, gdyby pan minister odpowiedział na nie na piśmie. Czy opracowano, czy wszystko zawiodło? Mój klub oczekuje wyjaśnienia tej sytuacji i podjęcia właściwych decyzji, w tym personalnych. Mówi pan, że uczelnia wprowadziła w błąd Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Ale pytam: Kto odpowiada za tę uczelnię? Samo powołanie komisji śledczej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej nie wystarczy. Dziś wiemy, że przez kontakt z podchorążymi jest zagrożonych kilkunastu kadetów ze szkoły pożarniczej w Poznaniu, bo przecież razem byli na poligonie w Drawsku. Czy zamierza pan, panie ministrze, zdymisjonować, jak myślę, odpowiedzialnego również w największej części rektora tej uczelni? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o udzielenie odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego. Wysoka Izbo! Przyszedłem tutaj nie po to, żeby występować, nie po to, żeby reagować na polityczne zaczepki, ale żeby przedstawić informację, bo jesteśmy w punkcie: Informacja w sprawach bieżących. Na podstawie waszych, szanowni państwo posłowie, pytań, można by odnieść wrażenie, że wszystko się wali, że służby nie funkcjonują itd. Nie, jest dokładnie. Szanowni państwo, teraz mówię do opinii publicznej i naszej. Wszystkie służby mundurowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych wykonują swoje zadania w 100%, a nawet więcej niż w 100%, w 200%. Policjanci, Straż Graniczna, straż pożarna wykonują naprawdę z ogromnym zaangażowaniem swoje zadania na rzecz obywateli w tym niezwykle trudnym czasie. Proszę mi nie przerywać, tak jak ja państwu nie przerywałem.

Proszę was o jakąś elementarną odpowiedzialność i lojalność państwową. Jesteście funkcjonariuszami publicznymi i waszym celem nie powinno być sianie plotek z trybuny sejmowej, kolportowanie jakichś absurdalnych, nieprawdziwych, niepokojących obywateli informacji. Pan, panie pośle, kilkakrotnie uczestniczył w spotkaniach w ostatnich tygodniach z przedstawicielami rządu jako przedstawiciel opozycji. Za każdym razem pytał mnie pan o rzekome braki środków dezynfekcyjnych na komendach Policji. Pytam pana o konkrety, o konkretne komendy. Podajcie mi przykłady. To wszystko nie jest prawda.

Traktuję to jako bardzo przykry incydent. Jest mi wstyd wobec podchorążych szkoły pożarniczej, że władza uczelni nie zachowała się wobec nich lojalnie, nie okazała im należytego zaufania. Jest powołana komisja, która wyjaśni wszystkie aspekty.

Prawda okazała się inna i konsekwencje będą wobec wszystkich wyciągnięte. Ja się niezwykle, mogę tylko to powiedzieć, cieszę, że żaden z podchorążych nie wymaga na dzień dzisiejszy hospitalizacji, i mam nadzieje, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdą obronna ręką z tej sytuacji, do której nie powinno było dojść, ale to jest sytuacja całkowicie jednostkowa. I cały szereg informacji szczegółowych, które tutaj w tych pytaniach czy pseudopytaniach padały, było nieprawdziwych. Oczywiście ustosunkujemy się na piśmie do tego wszystkiego. Następne testy będą jeszcze raz przeprowadzone w ciągu 5–7 dni. Wykryto 51 przypadków - jest to skala bardzo duża i niepokojąca - na 386 osób, wobec których testy przeprowadzono. Zaopiekujemy się tymi podchorążymi. To jest oczywiste zupełnie, to jest nasz obowiązek i nikt tu nikomu łaski nie robi. Pierwsza osoba z władz uczelni poniosła konsekwencje. Jest powołana komisja przez komendanta głównego. Nikt niczego nie będzie tu chował pod korcem. I informuję państwa, że to była moja pierwsza i jedyna póki co decyzja personalna jako ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego wobec władz tej uczelni. Ja tych ludzi nie powoływałem. Jeżeli będzie potrzeba, stracą następne. Jeśli uznamy, że są winni, że stchórzyli, że nie stanęli wobec tego wyzwania na wysokości zadania, nikt tu nie będzie nikogo ukrywał niezależnie od tego, kto, komu, czyj brat tam robił operację. Sytuacja jest naprawdę poważna i miejcie odpowiedzialność państwową również wobec obywateli, żeby tu głupot nie opowiadać. Wszystkie służby mundurowe są zabezpieczone i wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.

Wznawiam obrady. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Stwierdzam kworum. Informuję, że prezes Rady Ministrów zawiadomił Sejm o zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, poprawki w sprawie zmian klimatu, przyjętej w Lillafüred dnia 12 października 2017 r., do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. Posłowie w określonym terminie nie zgłosili zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Komisja Spraw Zagranicznych przedłożyła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie tego zawiadomienia premiera bez zastrzeżeń. W związku z tym, na podstawie art. 120 ust. 4 regulaminu Sejmu, informuję o braku zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie to druk nr 333. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że planowany punkt 11. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, druk nr 274, nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Pan poseł Piotr Adamowicz, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Żyjemy w dobie epidemii, która dotyka wielu współobywateli, a z powodów gospodarczych z pewnością dotknie znaczne rzesze naszego państwa. W związku z tym, na podstawie art. 184 ust. 3 pkt 1 uchwały Sejmu o regulaminie Izby, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia w celu rozpatrzenia wniosku o wycofanie z porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia Sejmu punktu obejmującego informację prokuratora generalnego - ministra sprawiedliwości na temat etapu, na jakim znajduje się postępowanie w sprawie zabójstwa na tle politycznym prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dwa słowa uzasadnienia. Są sprawy ważne, ale są sprawy pryncypialne, ekstraordynaryjne, a taki jest dzisiaj czas. Niewątpliwie to nie było typowe zabójstwo, to było świadomie zaplanowane morderstwo. Wniosek o informację prokuratora generalnego został złożony 3 miesiące temu. Przeleżał się. W związku z sytuacją składam wniosek o rozpatrzenie wycofania tego wniosku. Chciałam tylko wyjaśnić, że to będzie przedmiotem dzisiejszego głosowania, właśnie to. Tak że tego wniosku nie poddam pod głosowanie, bo to jest w porządku dzisiejszych obrad, panie pośle. Szczęść Boże! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dowiadujemy się o tym już bez żadnego zdumienia, ale kiwając głową, i przyjmujemy informację, że pani marszałek raczyła nie dopuścić żadnych pytań przed dzisiejszymi głosowaniami. Rozumiem, że pani marszałek potwierdza tę swoją decyzję. Zatem wnoszę o uzupełnienie porządku obrad, czego oczywiście trzeba by dokonać formalnie, zarządzając przerwę, zbierając Konwent Seniorów, po to, żeby mogli zabrać głos przynajmniej przedstawiciele wnioskodawców projektów obywatelskich obecni w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, państwo Kaja Godek, Robert Bąkiewicz i Mariusz Dzierżawski. Być może są jeszcze inni przedstawiciele wnioskodawców. Bardzo prosimy o to, żeby obywatele, setki tysięcy, łącznie to są liczby idące w miliony (Dzwonek), Polaków miały głos w tej sali w chwili, kiedy ważą się losy Polski, kiedy przegłosowane mają być. Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska - PSL - Kukiz15.

Wysoka Izbo! Mam prośbę, żeby pani marszałek, żebyśmy zarządzili przerwę, żeby pani marszałek zwołała Konwent, żebyśmy mogli szybko przeprocedować ustawę o bezpłatnym zapewnieniu maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców Polski. Maseczka jest najlepszym sposobem, nie szalik, tylko właśnie maseczka. Żeby mogło się to odbywać sprawnie w całym kraju, to obywatele po tej decyzji powinni mieć bezpłatny dostęp do takich maseczek. Dzisiaj wywiązują się z tego samorządy. Choćby w Lewinie Brzeskim Paweł Kukiz razem z burmistrzem, z samorządowcami dostarcza dzisiaj maseczki mieszkańcom. Tak się dzieje w wielu miejscach w Polsce. Ale to rolą państwa i rolą rządu jest (Dzwonek) zapewnienie bezpłatnych maseczek.

Wycofuje pan czy nie wniosek o przerwę, panie pośle? W takim razie przegłosujmy wniosek o przerwę.

Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę do góry.

Wniosek nie przeszedł. Jeszcze z wnioskiem formalnym pani poseł Katarzyna Lubnauer, Lewica. Proszę. Pani poseł Ueberhan, Lewica, przepraszam. Wysoka Izbo!

Wniosek oczywiście jest bezprzedmiotowy. Doskonale pani o tym wie. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 49, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. W dyskusji złożono wnioski: - o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, - o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania, bez odsyłania projektu do komisji. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 282, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest skierowanie tego projektu ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Pod głosowanie poddam wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy, bez odsyłania do komisji. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do komisji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 282, bez odsyłania do komisji, zechce nacisnąć

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 39, zechce nacisnąć

Na podstawie art. 87 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W dyskusji zgłoszono wnioski: o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 36, zechce

Sejm wniosek odrzucił. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest skierowanie tego projektu ustawy do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Pod głosowanie poddam wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy bez odsyłania do komisji. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do komisji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 36, bez odsyłania do komisji, zechce nacisnąć

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 251-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Wysoka Izbo! W drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zgłoszonych zostało siedem poprawek. To są poprawki dotyczące ujednolicenia daty wejścia w życie ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 251. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 2. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 6., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. W 3. poprawce wnioskodawcy proponują skreślenie art. 4 projektu ustawy nowelizującej. Z poprawką tą łączy się poprawka 7. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 3. i 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 5.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 251, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

447 - za, 5 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 272 i 333) Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 272. Marszałek Sejmu zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 18 marca 2020 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia.

Tak wnosi Komisja Infrastruktury. Dziękuję, pani poseł. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Z poprawką tą łączy się poprawka 6. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Przystępujemy do głosowania.

W 9. poprawce do załącznika do ustawy w tabeli nr 6 Senat proponuje nie zmieniać kolumny trzeciej. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Prawo budowlane Senat proponuje nie uchylać ust. 4. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Z wnioskiem formalnym pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Jeśli pani pozwoli, chciałbym złożyć wniosek formalny o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o informację prezesa Rady Ministrów w sprawie dramatycznej sytuacji placówek stałego pobytu w województwie mazowieckim i bezprawnych działań wojewody mazowieckiego. Pani Marszałek! Państwo, które nie potrafi chronić najsłabszych i najbardziej bezbronnych, nie potrafi chronić nikogo. Takiej ochrony i wsparcia nie zapewnia wojewoda mazowiecki. Pokazują to miejsca, gdzie pojawił się koronawirus, a wojewoda wyposażony w kompetencje ustawowe okazał się całkowicie bezradny. Tę nieudolność symbolizują takie miejsca, jak Bobrowiecka, Tomczyce, Niedabyl, Rusiec, Grójec czy też Radom. Druga sprawa, pani marszałek, to jest - odnoszę się teraz do pana premiera - kwestia bezprawnych działań związanych z nakazem pracy. Pan wojewoda Radziwiłł nie stosuje ustawy o chorobach zakaźnych. Nakazem pracy obejmuje osoby powyżej 60. roku życia, matki samotnie opiekujące się dziećmi oraz chociażby takie matki, jak pani, która w tej chwili jest na urlopie macierzyńskim, karmi 5-miesięczne dziecko. Na te osoby nakładane są 5-tysięczne kary. Ta sprawa bulwersuje, ponieważ mamy do czynienia z całkowitą nieudolnością wojewody mazowieckiego. Mam wrażenie, że pan wojewoda Radziwiłł zagraża w tej chwili bezpieczeństwu zdrowotnemu tego województwa. Panie Premierze! Prosimy o informację, o uzupełnienie porządku obrad. Pan wie doskonale, że to nie jest wniosek formalny.

Porządek dzienny był ustalony i dlatego tego wniosku nie mogę poddać pod głosowanie. Proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Otóż za chwilę będziemy głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad informacji rządu na temat kolejnego zagrożenia, które jest przed nami, a mianowicie kwestii związanych z klęską suszy. Niestety od 7 stycznia tego roku, gdy złożyliśmy ten wniosek, nie było żadnych konkretnych informacji ze strony rządu. To bardzo ważne, żeby zabezpieczyć Polaków przed tym, co może nadejść: suszą, ale również kwestiami wysokich cen żywności. W tej Izbie powinien stanąć minister klimatu i powiedzieć, w jaki kompleksowy sposób państwo chce walczyć ze skutkami być może największej od wielu lat suszy.

Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Informacja Ministra Klimatu na temat: - aktualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polaków wynikającego z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, tj. suszy, wzrostu średnich temperatur, nieprzewidzianych zjawisk pogodowych, zagrożenia pożarowego - na przykładzie bezprecedensowych pożarów w Australii, - uchybień w pracach nad stworzeniem oraz przedłożeniem opinii publicznej i właściwym organom Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2021–2030 oraz Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2021–2050 (tzw. strategia długoterminowa) - zgłoszona przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni; - Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac nad zwiększeniem świadczeń emerytalnych i rentowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwoty minimalnej emerytury i renty - zgłoszona przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia); - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwych nadużyć w dysponowaniu środkami pochodzącymi z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działań, jakie zostały podjęte w wyniku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, w szczególności udzielenia odpowiedzi, czy rzeczywiście została złożona oraz nieprzyjęta dymisja szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - zgłoszona przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni; - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat wyprowadzenia znaczącej kwoty pieniędzy z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz niewłaściwego sprawowania nadzoru nad tą służbą - zgłoszona przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia); - Informacja Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów na temat działań podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sprawie restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku - zgłoszona przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni; - Informacja Ministra Finansów w sprawie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i działań KNF - zgłoszona przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji ministra klimatu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji na temat prac nad zwiększeniem świadczeń emerytalnych i rentowych.

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji na temat możliwych nadużyć w dysponowaniu środkami pochodzącymi z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji na temat wyprowadzenia znaczącej kwoty pieniędzy z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji na temat działań podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sprawie restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji na temat przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i działań KNF. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił.

Pani poseł, ja bym raczej prosiła, żeby apelować do Senatu.